Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. Skala i natężenie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego przetaczających się przez Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich, które odbyły się w sierpniu 2020 r., wymagają solidarności i zdecydowanych działań społeczności międzynarodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowanie potępia akt terroru państwowego polegający na doprowadzeniu do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r., co stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego oraz bezprawne zatrzymanie przez białoruskie władze Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Żądamy ich natychmiastowego uwolnienia oraz zagwarantowania im swobody przemieszczania się. Zwracamy się do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne zbadanie tego bezprecedensowego i niedopuszczalnego zdarzenia. Apelujemy do parlamentów krajów Unii Europejskiej i Rady Europy o aktywne i wspólne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi, a także o wzmacnianie solidarnego stanowiska państw europejskich wobec reżimu w Mińsku, w szczególności o wspieranie działań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych i powstrzymania represji. Apelujemy do Rady Ministrów o złagodzenie zasad polskiej polityki azylowej i polityki udzielania ochrony międzynarodowej wobec białoruskich uchodźców politycznych. Z niepokojem oceniamy eskalację represji skierowanych przeciwko społeczeństwu białoruskiemu, których kolejne sekwencje doprowadziły do dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się także nasi Rodacy, obywatele Białorusi żyjący od pokoleń na tej ziemi. Kulminację tych wydarzeń stanowi aresztowanie Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewskiej, Marii Tiszkowskiej i Ireny Biernackiej. Żądamy jak najszybszego uwolnienia osób zatrzymanych i zaprzestania stosowania wobec nich represji łamiących podstawowe prawa człowieka. Popieramy konkluzje nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej i apelujemy o jak najszybsze rozszerzenie wykazu sankcyjnego o dodatkowe osoby i podmioty, a także o ukierunkowane sankcje gospodarcze wobec reżimu. Apelujemy również do Rady Ministrów o zdecydowane, konsekwentne i konkretne działania w tej sprawie, w tym objęcie sankcjami osób aparatu władzy, sprawiedliwości i bezpieczeństwa biorących bezpośredni udział w represjach wobec Polaków na Białorusi”

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. Panie pośle, przepraszam bardzo, wnioski formalne. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę informacji na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. Od ponad tygodnia jesteśmy świadkami politycznego ping-ponga pomiędzy polskim a czeskim rządem, wymiany zdań, której dałoby się uniknąć, gdyby strona polska od początku usiadła do stołu i podjęła rozmowy. Rząd próbuje teraz bohatersko rozwiązać problem, który sam stworzył.

Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Drugi wniosek formalny - pan poseł Stanisław Żuk, Kukiz’15. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! W styczniu 1958 r. Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy kompleksu Turów. Inwestycja polegała na budowie elektrowni o mocy 1200 MW i rozbudowie kopalni Turów. Dzisiaj mamy sytuację nadzwyczajną. Po 32 latach istnienia niepodległej i demokratycznej Polski jednoosobowo wiceprzewodnicząca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 21 maja 2021 r. podjęła decyzję o wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Jest to decyzja nieuzasadniona, uderzająca w niezależność energetyczną Polski i naszą niepodległość polityczną. Takie postanowienie rodzi ogromnych rozmiarów skutki społeczne i gospodarcze.

Dziękuję panu bardzo. To nie jest wniosek formalny. To proszę od tego zaczynać, panie pośle. Nie słyszę, pani marszałek.

Przykro mi.

Zgłaszam wniosek o odroczenie obrad, wspierając pana posła Żuka w tym, że dzisiaj Sejm powinien natychmiast wydać uchwałę o tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma prawa do tego, żeby zamykać nam kopalnię, likwidować nam energetykę. To jest nasz interes narodowy. To jest oczywiście kamyczek do ogródka lewej strony sali, tej rządzącej również, pokazujący, co oznacza przekazywanie kompetencji do Brukseli, to przekazywanie kompetencji, na które również Morawiecki zgodził się w ubiegłym roku. Tak to się właśnie kończy. Tak się kończy wyprzedawanie suwerenności przez Millera, przez Tuska i przez Morawieckiego - tym, co w Turowie. To jest wasza wspólna sprawka. To jest wasza wspólna sprawka, która zostanie rozliczona.

Jeszcze raz informuję, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu będzie informacja w tej sprawie. Turów leży w moim okręgu, więc też jestem żywo zainteresowana, żeby to się jak najszybciej skończyło, żeby mieszkańcy mogli spokojnie pracować, żyć i nie martwić o to, co będzie jutro. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Zgłaszam wniosek formalny, aby na debatę na temat Turowa i tego bezprecedensowego ataku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polską niezależność energetyczną zaprosić do Sejmu przedstawicieli wszystkich czterech central związkowych, którzy we Wrocławiu przed Komisją Europejską jasno powiedzieli: ręce precz od Turowa. To właśnie te centrale związkowe bronią dzisiaj polskiej niezależności energetycznej, bronią polskich miejsc pracy - i należy się im szacunek - za co im bardzo serdecznie dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1159 i 1165) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1165 i 1159.

Senat zgłosił 44 poprawki.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Głosujemy.

Kto jest przeciw?

Głosowało 449 posłów. W 4. poprawce do m.in. art. 170 ustawy - Prawo upadłościowe Senat proponuje nowe brzmienie ust. 7. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Senat proponuje we wprowadzeniu do wyliczenia inny termin wejścia w życie ustawy. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, 454 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Senat zgłosił do art. 2 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy - Prawo upadłościowe. W 10. poprawce do art. 19 ust. 4 Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjnym. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

1 - za, przeciw - 451, nikt się nie wstrzymał. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nikt nie był za, przeciw - 451, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 37. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1161 i 1180) Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie jest zawarte w druku nr 1180. Senat do tej ustawy wprowadził 24 poprawki. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpoznaniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 19 maja rekomenduje, aby Wysoki Sejm raczył 13 poprawek przyjąć i 11 odrzucić.

W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej z druku nr 1211, którą to uchwałę pani marszałek skierowała do Komisji Spraw Zagranicznych dnia 27 maja br. w celu rozpatrzenia. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych uchwałę rozpatrzyła. Komisja wnosi, by Wysoki Sejm raczył poprawkę Senatu odrzucić. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1176-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw złożono 10 poprawek. Zostały one ponownie skierowane do Komisji Infrastruktury, która rozpatrzywszy te poprawki szczegółowo, rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucić poprawki od 1. do 9., przyjąć poprawkę 10. i oczywiście przyjąć całość projektu ustawy ze sprawozdania komisji, druki nr 1176 i 1176-A. Bardzo dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1176. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy.

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1176, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1204-A. Proszę panią poseł Lidię Burzyńską o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, druk 1204-A. Komisja rozpatrzyła wnioski i poprawki zgłoszone w drugim czytaniu i rekomenduje odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, odrzucenie wszystkich poprawek i prosi Wysoki Sejm o uchwalenie projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1204. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki? Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1204, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 40. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1205. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1205, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 41. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1208-A. Proszę pana posła Bolesława Piechę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek!

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1202. Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki 1. i 2. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 3. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie załącznika do ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 5. do 13. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 5. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują zmiany w liczbach porządkowych od 1 do 8. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 6. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują zmiany w liczbach porządkowych od 1 do 3 oraz od 6 do 8. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 7., 9. i 13. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

W 7. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują zmiany w liczbach porządkowych od 1 do 3. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 8. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują zmiany w liczbach porządkowych od 9 do 11. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 13. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 13. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 11. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują nowe brzmienie tytułu w kolumnie drugiej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 12. poprawce do załącznika do ustawy wnioskodawcy proponują nowe brzmienie tytułu w kolumnie drugiej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1202, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 43. porządku dziennego: Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 1139 i 1151) Wysoka Izbo!

Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pana Wojciecha Polaka w celu przedstawienia kandydatury. Bardzo proszę, panie profesorze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań, po przeanalizowaniu przedstawionych przez nich dokumentów i po długich naradach kolegium jednomyślnie uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Karol Nawrocki, obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W związku z tym przypada mi zaszczyt zgłoszenia i przedstawienia Wysokiej Izbie kandydatury dr. Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na tej uczelni uzyskał także stopień doktora nauk humanistycznych. Po studiach przez wiele lat pracował w oddziale gdańskim Instytutu Pamięci Narodowej na odpowiedzialnych stanowiskach. Od kwietnia 2017 r. jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Warto zresztą wspomnieć o jego osiągnięciach na tym stanowisku, np. o wystawie „Fighting and Suffering” - walka i cierpienie, zgodnie uznanej za największą w historii akcję polskiej dyplomacji historycznej. Wystawa została przetłumaczona na 37 języków i została pokazana w 160 miejscach na świecie. Dr Karol Nawrocki jest autorem lub współautorem kilku publikacji książkowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych z zakresu historii opozycji antykomunistycznej, historii sportu oraz przestępczości zorganizowanej w PRL. Jest także osobą zaangażowaną w utrwalanie pamięci historycznej w przestrzeni publicznej Pomorza. Jest członkiem kilku rad programowych znaczących polskich muzeów. Szczególnie ważne także w kontekście IPN są Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej w Warszawie, Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie czy Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Markowej. Jest członkiem Rady Dyplomacji Historycznej przy MSZ i członkiem Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Swoją koncepcję funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zawarł w słowach: prawda nie obroni się sama, sygnalizując tym samym potrzebę obrony prawdy dotyczącej historii Polski w kraju i za granicą w sposób usystematyzowany i konsekwentny. Z tak postawionego celu wynika zobowiązanie do koniecznej po 20 latach funkcjonowania IPN głębokiej refleksji dotyczącej kształtu organizacyjnego instytutu. Celem tej refleksji jest podniesienie efektywności działań urzędu zatrudniającego przecież 2,5 tys. osób. W koncepcji dr. Karola Nawrockiego obok utrzymania dotychczasowej dynamiki statutowych działań instytutu mieści się także wiele przedsięwzięć na płaszczyźnie międzynarodowej. Do najważniejszych można zaliczyć choćby szeroki projekt dotyczący instytucjonalnego wsparcia dla polonijnych archiwów i fundacji rozsianych po całym świecie czy - co uznał za jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata - przygotowanie naukowych i popularnonaukowych opracowań dotyczących zbrodni niemieckich i sowieckich w czasie II wojny światowej. Opracowania takie zostałyby przetłumaczone na wszystkie języki kongresowe.

Zadaniem nowego biura stanie się także dalsza cyfryzacja zasobu IPN i stworzenie możliwości do korzystania z niego w sieci. Dr Karol Nawrocki zapowiedział potrzebę kontynuowania prac badawczych i ekshumacyjnych polskich bohaterów, proponując poszerzenie zasięgu ekshumacji o Azję Środkowo-Wschodnią. Kolegium IPN wysoko oceniło te i inne projekty zaproponowane przez dr. Karola Nawrockiego.

Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Asta w celu przedstawienia opinii komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą wniosku Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o powołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr. Karola Nawrockiego. Komisja rozpatrzyła wniosek kolegium w dniu 14 maja 2021 r. i po wysłuchaniu kandydata i przeprowadzeniu dyskusji postanowiła zaopiniować tę kandydaturę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Ponieważ zgłosili się posłowie do zabrania głosu, proponuję, aby Sejm wysłuchał w dyskusji 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.

Po pierwsze, chciałbym wyrazić zdziwienie, że kandydat na stanowisko prezesa IPN nie siedzi na galerii, gdzie jest miejsce dla kandydatów, ale siedzi w tej chwili na fotelu [[Oklaski]] organu konstytucyjnego. Wysoka Izbo! Gdy PiS w końcu straci władzę, pośród wielu dylematów stojących przed przyszłym Sejmem pojawi się ten.

Gdy PiS w końcu straci władzę, pośród wielu dylematów stojących przed przyszłym Sejmem pojawi się też ten, co zrobić z instytucjami, które w ostatnich 5 latach uległy tak głębokiej degeneracji, że trudno uwierzyć, by dało się je w obecnym kształcie uratować. Niewiele zostało z autorytetu, jakim cieszyła się ta instytucja, gdy kierował nią pierwszy prezes prof. Leon Kieres. Ostatnie 5 lat funkcjonowania IPN to czas od kryzysu do kryzysu, od nowelizacji ustawy o IPN do nominacji hajlującego nacjonalisty, którego do końca bronili niektórzy politycy siedzący po tej stronie sali. Tylko ta sprawa potwierdza, że przedstawiciele skrajnej prawicy czuli się tam jak ryby w wodzie, robiąc szybkie i błyskotliwe kariery. Przejdźmy do kandydata. Kim jest pan dr Nawrocki? To przede wszystkim nominat tej władzy już raz użyty do przejęcia przez PiS jednej instytucji. Posłużył do odsunięcia prof. Pawła Machcewicza. Polityczna decyzja o przejęciu Muzeum II Wojny Światowej zapadła na Nowogrodzkiej. Doprowadził do zmiany wystawy głównej wbrew woli jej twórców. Szanowni Państwo! Również zaskakuje ostatni fakt.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Lewicy w sprawie kandydata na prezesa IPN-u. I od razu mówię: Lewica oczywiście będzie głosować przeciwko tej kandydaturze. Będziemy głosować przeciwko tej kandydaturze z dwóch powodów: po pierwsze, z powodu osoby kandydata, która jest niezwykle kontrowersyjna, a po drugie, dlatego że uważamy, że IPN należy zlikwidować. Jeśli chodzi o kandydata - to kandydatura niezwykle kontrowersyjna.

Oczywiście nie wolno nie wspomnieć o tym, jak pod dyktando PiS-u pan Nawrocki zmieniał wystawę stałą w Muzeum II Wojny Światowej.

To znacznie więcej niż roczny budżet Państwowej Inspekcji Pracy czy rzecznika praw obywatelskich. Lewica złożyła kilka tygodni temu projekt ustawy likwidującej IPN.

Tym będzie zajmował się ten instytut. Natomiast prokuratorzy pracujący w IPN-ie zostaną przeniesieni do prokuratury. Wysoka Izbo! Bardzo proszę panią marszałek o rozpoczęcie.

Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! W życiorysie, w dorobku naukowym, zawodowym pana doktora faktycznie można znaleźć wiele akcentów, które były niezwykle kontrowersyjne, ale też gdyby bliżej przyjrzeć się temu dorobkowi, można znaleźć również inicjatywy, którym trudno odmówić słuszności i wartości. Dzisiaj na tej sali, Wysoka Izbo, wydaje się, kwestia głosowania jest przesądzona. O wyborze prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zdecyduje głosowanie na forum Senatu. Ja w imieniu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, panie doktorze, bardzo chętnie podjąłbym np. rozmowę w naszym klubie na temat rehabilitacji Wincentego Witosa, który mimo tylu lat nie może doczekać się przywrócenia właściwego miejsca w pamięci i w historii Polski.

Sfera kadrowa, sfera całego otoczenia, które faktycznie nie najlepiej się miewa w ostatnich latach, jest też oczywiście istotną dziedziną, ale chcielibyśmy przede wszystkim o przywracaniu pamięci wielu ważnych postaci, w tym Wincentego Witosa... Korfantego. Proszę. Wysoka Izbo! Karol Nawrocki to może być dobry kandydat. To może być naprawdę dobry kandydat. Biorąc pod uwagę to, co zrobił z Muzeum II Wojny Światowej, ja jestem dobrej myśli. Ale tutaj też jest dobry moment na to, by powiedzieć o tym, co należy jeszcze zrobić w Instytucie Pamięci Narodowej.

IPN powinien zdecydowanie zająć się także obroną dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej, ponieważ wiemy, że jesteśmy atakowani od dziesiątków lat, są kręgi, którym nie podoba się to, jak naprawdę wyglądała nasza historia, które robią z nas antysemitów, robią z nas żydożerców, robią z nas ludzi, którzy nie są cywilizowani. A to nie jest prawda.

To też jest zadanie dla IPN-u. Czyli to praca nad młodzieżą, nad młodym pokoleniem, ponieważ ostatnie lata to była faktycznie bardzo merytoryczna praca, natomiast praca, która nie trafiała do młodych ludzi. Nad tym warto się zastanowić.

Wysoki Sejmie! Sprawozdanie komisji to tylko suchy komunikat. Kandydat Karol Nawrocki zyskał niewielkie poparcie w komisji sprawiedliwości. Informuję o tym, bo jak mówi kandydat na nowego prezesa IPN, prawda nie obroni się sama. Podczas posiedzenia komisji kandydat zapowiedział wdrożenie nowych technologii pozwalających na skuteczny międzypokoleniowy dialog. Działanie Instytutu Pamięci Narodowej miałoby być przekładane na język gier komputerowych. Kandydat zapowiedział aktywność na polu kultury, bo jego zdaniem można edukować poprzez koncerty czy sztuki teatralne. Gry niech tworzą specjaliści, koncerty niech organizują fachowcy, sztuki niech wystawiają niezależni twórcy, niepodporządkowani nikomu i niedziałający na niczyje zlecenie. Bo prawda obroni się sama.

Polska 2050 nie poprze kandydatury Karola Nawrockiego, choć cieszy nas, że lubi sport - uprawia boks. Nie popieramy jednak tego, by muzeum, którym kierował do tej pory, było partnerem komercyjnych walk bokserskich. Lepiej popularyzować boks, sport, jego historię, choćby pokazując sylwetkę pierwszego po wojnie złotego medalisty olimpijskiego Zygmunta Chychły.

Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za powołaniem pana Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zechce nacisnąć

Sejm powołał pana Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Gratuluję. O głos poprosił wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pan Piotr Gliński.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Bardzo się cieszę z tego głosowania, z wyniku tego głosowania, bo współpracuję z panem dr. Karolem Nawrockim od kilku lat i mogę mówić o tej współpracy tylko w samych superlatywach. To jest osoba odpowiedzialna, kompetentna, odważna. Jednak w związku z pewnym wątkiem, który był tutaj poruszany w trakcie dyskusji, z krzywdzącymi i niegodnymi pomówieniami dotyczącymi zmian, jakie musiały być dokonane w ekspozycji stałej Muzeum II Wojny Światowej, chciałem Wysokiej Izbie przedstawić, czego te zmiany dotyczyły, gdyż to mówi wszystko zarówno o kandydacie, jak i o dylemacie, jaki mamy w Polsce z polityką historyczną i rozumieniem prawdy historycznej. Najlepiej przedstawić ten dylemat i treść tych zmian poprzez treść pozwu złożonego przez poprzednią dyrekcję tego muzeum, której przewodniczył pełnomocnik premiera Tuska do spraw budowy owego muzeum.

W punkcie pierwszym żądano usunięcia z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej portretu o. Maksymiliana Marii Kolbego wraz ze stanowiskiem multimedialnym. W punkcie drugim - usunięcia z wystawy głównej portretu Witolda Pileckiego. W punkcie trzecim - usunięcia z wystawy głównej zdjęcia powstańców warszawskich składających przysięgę wojskową. usunięcia z wystawy głównej zdjęcia rodziny Ulmów wraz ze stanowiskiem multimedialnym.

W punkcie ósmym - usunięcia z wystawy głównej ekspozytora poświęconego mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” W punkcie dziewiątym - usunięcia z wystawy głównej ekspozytora poświęconego Marianowi Rejewskiemu.

W punkcie jedenastym - usunięcia z wystawy głównej.

Jak państwo może pamiętacie, w pierwotnej wersji wystawy stałej polska partyzantka była zrównywana z francuską w owym czasie. W punkcie czternastym - usunięcia z wystawy głównej statystyk strat osobowych, usunięcia z wystawy głównej produkcji IPN-u „Niezwyciężeni”, to taka pamiętna krótka produkcja, która mówiła o naszym rozumieniu historii. Przywrócenia pierwotnej formy scenograficznej wystawy w części poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu. I wreszcie w siedemnastym punkcie - przeniesienia eksponatów dotyczących kpt. Antoniego Kasztelana w pierwotne miejsce ich prezentacji, czyli do gabloty z eksponatami dotyczącymi Rudolfa Spannera. Tak wyglądały te zmiany, tylko podstawowe, ograniczone w swojej treści.

Panie premierze, bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 45. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1220)

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1220, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Ogłaszam 2 minuty przerwy.

Wznawiam obrady. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zabrać głos, dopisać się do listy? Jeśli nie, to listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam za zamkniętą.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uważam, że jest to nieuzasadniona decyzja uderzająca w niezależność energetyczną Polski oraz w bezpieczeństwo miejsc pracy i źródeł utrzymania dla tysięcy mieszkańców tego regionu. Tak daleko sięgającą ingerencję w życie gospodarcze Polski należy zakwestionować. Rząd polski nie uzasadnił wyczerpująco faktu, że ewentualne wstrzymanie prac przez kompleks Turów doprowadzi do załamania dostaw energii elektrycznej dla polskiej gospodarki. Apeluję do rządu polskiego o podjęcie rzeczowych rozmów ze stroną czeską w celu wypracowania wspólnego kompromisu w kwestii kopalni Turów. Spór między Polską a Czechami został już nagłośniony w całej Europie. Sposób, w jaki Polska zareaguje na tę krzywdzącą nas decyzję, będzie miernikiem oceny dyplomacji naszego kraju. Przez całe życie zawodowe byłem związany z sektorem górniczym i energetycznym. Znam doskonale mechanizmy funkcjonowania tego rynku. Wiem dobrze, w jakich warunkach geologicznych, gospodarczych, środowiskowych pracuje kopalnia Turów. Oświadczam, że deklaruję pomoc i wsparcie dla wszystkich, którym na sercu jest spokojna i bezkonfliktowa praca kopalni i elektrowni Turów w celu rozwiązania sporu z Republiką Czeską. Cel jest jeden - wypracowanie optymalnych rozwiązań zabezpieczających funkcjonowanie kompleksu Turów jako niezbędnego elementu krajowego systemu energetycznego zgodnie z przyjętymi wiele lat temu planami. Dziękuję. Proszę teraz pana posła Jana Szopińskiego, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego w województwie kujawsko-pomorskim i miejscowości leżących pomiędzy Sępólnem a Bydgoszczą zostali zaskoczeni w kwietniu br. wiadomością o zawieszeniu przez PKS Chojnice wszystkich połączeń autobusowych z Chojnic do Bydgoszczy przez powiat sępoleński. Tym samym mieszkańcy ci zostali pozbawieni jedynego środka transportu do administracyjnej stolicy województwa kujawsko-pomorskiego, do bydgoskich szpitali specjalistycznych, w tym do takich szpitali i usług, których na terenie powiatu sępoleńskiego nie ma, czyli do pulmonologii, szpitala zakaźnego czy szpitala onkologicznego. Mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości dojazdu do urzędu wojewódzkiego i zostali pozbawieni możliwości dojazdu do portu lotniczego.

Niestety, marszałek odmówił samorządowcom i mieszkańcom, którzy kolejny raz poczuli się pozbawieni przez władzę możliwości kontaktu i zostali pozbawieni transportu. Jako poseł wybrany również przez mieszkańców powiatu sępoleńskiego zwracam się do rządu z postulatem wykorzystania wszystkich możliwych środków i programów rządowych, by przywrócić połączenia autobusowe pomiędzy Sępólnem Krajeńskim a Bydgoszczą i dbać o nie tak samo jak o pozostałe połączenia komunikacyjne w innych częściach naszego kraju. Zwracam się do ministra infrastruktury, do całego rządu o rzeczywiste, a nie tylko propagandowe i fasadowe działanie w celu zastopowania m.in. takich wykluczeń komunikacyjnych. Dziwne, że rząd, który powołał Polską Agencję Kosmiczną w celu narodowego podboju kosmosu, który buduje największe lotnisko w Europie, nie potrafi skutecznie załatwić tak prostej sprawy jak zapewnienie tego, by można było przewozić mieszkańców z miejscowości do miejscowości. Dlatego w imieniu mieszkańców powiatu sępoleńskiego raz jeszcze apeluję do rządu o takie działania, by zapewnić mieszkańcom powiatu (Dzwonek) sępoleńskiego połączenia autobusowe pomiędzy Sępólnem Krajeńskim a Bydgoszczą. Tymczasem proszę o wygłoszenie oświadczenia pana posła Sławomira Skwarka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W tym roku mija dokładnie 475 lat od nadania przez króla Zygmunta Starego przywileju lokacyjnego miastu Stoczek Łukowski. Historycznie Stoczek położony jest w ziemi czerskiej na Mazowszu, geograficznie - na Wysoczyźnie Żelechowskiej, a administracyjnie jest obecnie gminą miejską w powiecie łukowskim w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, jedną z najmniejszych gmin w Polsce. Obecnie w Stoczku mieszka ok. 2700 mieszkańców dumnych z historii swojego miasta. Miejscowość nosiła kilka nazw, m.in. Wola Poznańska, Sebastianowo. Od XVII w. znana jest pod obecną nazwą. W swojej historii po utracie niepodległości miasto znajdowało się pod zaborem austriackim, w Księstwie Warszawskim, w Królestwie Polskim, a następnie pod zaborem rosyjskim. W 1867 r. w ramach represji po upadku powstania styczniowego Stoczek został pozbawiony praw miejskich. Odzyskał je w roku 1916. Stoczek Łukowski znany jest przede wszystkim z pierwszej zwycięskiej bitwy powstania listopadowego. Wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego rozgromiły rosyjski korpus gen. Geismara. W Stoczku 18 stycznia 1849 r. urodził się Aleksander Świętochowski, pisarz, publicysta, krytyk, ideolog, konserwatysta epoki pozytywizmu. W okresie międzywojennym odbywały się tu największe w Polsce targi końskie i jedne z większych w Europie. Można powiedzieć: tych targów z końmi mi żal. Obecnie najważniejszą imprezą kulturalną jest organizowany Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, a sportową - odbywający się od 2001 r. bieg uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty” W związku z przypadającą rocznicą samorząd miasta we współpracy z instytucjami i partnerami społecznymi przygotował cykl imprez mających przybliżyć wydarzenia związane z historią miasta. W dniu 12 czerwca odbędzie się uroczysta sesja rady miasta.

W związku z rocznicą nadania prawa miejskiego mieszkańcom grodu z kogutem, miastu walki i oręża, życzę władzom samorządowym śmiałych wizji rozwoju, realizacji zamierzeń zawsze w oparciu o historię, kulturę i tradycję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje wystąpienie będzie dotyczyć Polskiego Bonu Turystycznego.

Ten program miał obowiązywać przez 2 lata. Proszę zobaczyć, że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o koronakryzys, koronawirus zaatakował na tyle poważnie, że wyłączone zostały wszelkie jednostki turystyczne, jeżeli chodzi przynajmniej o hotele, które miały dostać dofinansowania, z których miało skorzystać ponad 6 mln dzieciaków. Tutaj ten program nie do końca spełni oczekiwania polskich obywateli, bo może obowiązywać jeszcze tylko przez rok. Wystosowałem w tej sprawie interpelację do pana wicepremiera Jarosława Gowina, ponieważ on odpowiada za resort, który mógłby dokonać zmian w tej ustawie. Natomiast wystosowałem też prośbę o wsparcie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo wiem, że to był bardzo ważny programowo punkt w jego kampanii wyborczej. Myślę, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o przedłużenie obowiązywania tego bonu przynajmniej do 2023 r., do marca, może spowodować, że rozłożymy możliwość skorzystania z tego świadczenia.

Tak że podczas tego wystąpienia proszę pana wicepremiera Gowina, aby pochylił się nad tym programem, nad rozszerzeniem tego programu. Proszę również pana prezydenta Andrzeja Dudę, aby przychylił się do pozytywnej rekomendacji, aby ten projekt mógł zafunkcjonować rok dłużej, aby wydłużyć obowiązywanie tego projektu.

Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę pana posła Dariusza Olszewskiego o wygłoszenie oświadczenia. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiązując do mojego wystąpienia w Sejmie w dniu 2 marca ub.r., ponownie apeluję do władz Rzeczypospolitej Polskiej, do przedstawicieli rządu i parlamentu, o podjęcie odważnych i zdecydowanych działań zmierzających do właściwego uhonorowania żołnierzy wyklętych, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy do końca byli wierni swojej ojczyźnie, oraz wszystkich poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę. Wzywam do otoczenia szczególną troską wszelkich miejsc zroszonych krwią i oznaczonych cierpieniem żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Ich oprawcy powinni być jednoznacznie wskazani, a jeśli byłoby to także możliwe, również ścigani. Wspieranie działań zmierzających do poszukiwania prawdy historycznej i odkrywanie miejsc tajnych pochówków ofiar reżimu komunistycznego winno być naszym zobowiązaniem. Bohaterowie narodowi powinni powrócić na karty polskiej historii z imieniem i nazwiskiem. Ich szczątki muszą być podjęte z bezimiennych dołów, zidentyfikowane i złożone z należnymi im honorami w godnym tego miejscu. Niechlubnym przykładem przewlekania działań i braku odważnych decyzji jest sprawa kwatery Ł Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Z tego miejsca apeluję i proszę, aby miejsce tajnych pochówków na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach, terenie kwatery Ł, stało się prawdziwym narodowym panteonem pamięci. Już czas, aby powstał tam pomnik pamięci i wdzięczności za poświęcenie, krzywdę i cierpienie, jakie spotkało obrońców polskości, aby było to miejsce godne wolnej i niepodległej Polski. Teren łączki sąsiaduje niemal bezpośrednio z pomnikiem i grobami ofiar katastrofy smoleńskiej. Rozpoczyna się tam jedna z alei zasłużonych. To czyni ten rejon cmentarza głównym miejscem wielu uroczystości i stałym, obowiązkowym punktem wielu wycieczek oraz lekcji historii. Uzupełnieniem tego miejsca i przyszłego narodowego miejsca pamięci winna być nowa główna brama wybudowana od strony południowo-zachodniej. Po jej przekroczeniu każdy odwiedzający to miejsce, rozpoczynając zwiedzanie, mógłby w pierwszej kolejności skłonić głowę przed tymi, o których z woli władzy komunistycznej polska miała zapomnieć. Jako naród winni jesteśmy naszym bohaterom szczególną wdzięczność i systematyczną opiekę nad ich grobami, a w przypadkach znieważenia - skuteczną ochronę symboli i obronę pamięci, w tym także na drodze prawnej. Powody ewentualnych trudności i kłopotów przy realizacji tych celów należy niezwłocznie usunąć, tak w zakresie przepisów, jak i w sferze wykonawstwa. Cześć i chwała bohaterom! Bardzo dziękuję panu posłowi. Zapraszam panią poseł Annę Ewę Cicholską, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze od kilkudziesięciu lat wybory samorządowe. Były to zarazem pierwsze w III Rzeczypospolitej w pełni wolne wybory. Polska ma jedną z najdłuższych w Europie tradycji samorządu terytorialnego. Warto przypomnieć, że już w średniowieczu istniał system urzędów lokalnych i sejmików. System pełnił ważna rolę w funkcjonowaniu ówczesnego państwa. Ciągłość istnienia samorządu terytorialnego została zerwana wraz z upadkiem Rzeczypospolitej w 1795 r. Po odzyskaniu niepodległości praktycznie natychmiast podjęto działania w celu odbudowy struktur samorządu terytorialnego.

Po wojnie władze komunistyczne na krótko przywróciły samorząd terytorialny, ale wraz z postępującą sowietyzacją systemu politycznego przystąpiono do jego likwidacji. W marcu 1950 r. samorząd terytorialny przestał istnieć. Jego miejsce zajęły rady narodowe. 27 maja 1990 r. Polacy wybrali swoich przedstawicieli do rad miast i gmin. Wiele z moich koleżanek i kolegów w Sejmie ma doświadczenie w pracy w samorządach. Praca w samorządzie terytorialnym pomaga mi obecnie w sprawowaniu mandatu poselskiego. Nie powinniśmy zapominać, że samorząd terytorialny działa w ramach państwa. Samorząd to wspólnota lokalna, która otrzymała daleko idące uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach, które jej bezpośrednio dotyczą, ale trzeba pamiętać, że za te decyzje jest w pełni odpowiedzialna. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania zlecone przez administrację publiczną, wykonują również zadania własne, które są ważne dla wspólnot gminy, miasta czy województwa. Co ważne, zadania te nie mogą mieć charakteru i znaczenia ogólnokrajowego. Zarówno pierwsze, jak i drugie zadania wymagają sporych nakładów finansowych [[Dzwonek]] ze środków własnych samorządu i wsparcia rządowego. Wszystkim państwu samorządowcom życzę satysfakcji z działania na rzecz swoich lokalnych wspólnot. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę pana posła Mariusza Goska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Opozycja od 2 dni żyje odgrzewanym tematem związanym z wyborami na urząd prezydenta w Pretekstem i okazją do tego są ostatnie wypowiedzi pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Z tego miejsca warto przypomnieć, słysząc te medialne wypowiedzi, że to przecież opozycja twierdziła, że wybory nie powinny odbywać się w maju, tylko na jesieni. Jak malała, to wszyscy doskonale widzieliśmy: byliśmy w szczycie zachorowań. Nigdy ich nie przedstawił. Wszyscy doskonale o tym wiemy, bo taki stan faktyczny później się ujawnił. Obowiązkiem organów państwa było przeprowadzenie wyborów na urząd prezydenta w terminie konstytucyjnym. Działania dokładnie w takim kierunku zostały podjęte przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia.

Jak można było podejmować działania w takim kierunku, żeby urząd prezydenta był nieobsadzony i to stanowisko było stanowiskiem wakującym?

Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia panią poseł Klaudię Jachirę, Koalicja Obywatelska. Panie przewodniczący komitetu do spraw bezpieczeństwa Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po co tak kłamiecie?

Dużo prościej, tak jak dzisiaj na sali sejmowej, jest przyjąć uchwałę, niż realnie pomóc Białorusinom. Jak to możliwe, że jednego prezesa partii rządzącej chroni u nas 40 policjantów przez całą dobę, a przecież nie robi on nic ważnego, a ludziom, którzy narażają się i walczą z reżimem o wolną ojczyznę, którzy często spotykają się z groźbami karalnymi, nie zapewnia się polskiej ochrony? Swoją drogą, jak premier Kaczyński się tak boi, to może nie powinien odpowiadać za bezpieczeństwo innych. Doszło do tego, że dla Białorusinek i Białorusinów mała Litwa staje się dobrą matką, a Polska jak macocha nie potrafi ich pokochać i po ludzku im współczuć. Przecież ci ludzie chcą u nas pracować, płacić podatki, uczyć się, a każda sprawa, którą próbują załatwić, wiąże się dla nich z ogromną biurokracją i staniem godzinami w kolejkach do urzędów.

Niech żyje wolna Białoruś! Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę pana posła Michała Urbaniaka o wygłoszenie oświadczenia.

Wysoka Izbo! Wychodzę dziś z apelem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana premiera Glińskiego oraz do sekretarza stanu pana Jarosława Sellina. Otóż niemal 40 lat temu mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego wraz z proboszczami parafii Podwyższenia Krzyża Świętego domagali się zwrotu ołtarza antwerpskiego z 1550 r., który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie jako ołtarz skrzydłowy, tryptyk z tej właśnie parafii.

W 1990 r. ta decyzja została podtrzymana przez ówczesną minister kultury i sztuki panią Izabellę Cywińską. Ona poleciła dyrektorowi muzeum zwrot w trybie pilnym. Niestety to polecenie nie zostało wykonane, natomiast zarówno ze strony parafii, jak i miasta nałożone warunki zostały spełnione. Sytuacja jest nierozwiązana.

W 2016 r., bo sprawa trwa, jak powiedziałem, bardzo długo, senator RP pan Antoni Szymański, notabene wtedy właśnie też z partii rządzącej, pytał o to i dowiedział się, że na podstawie komunistycznych dekretów nie ma takiej możliwości, by ten ołtarz wrócił do Pruszcza, że stał się on własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ten ołtarz jest ważny dla Pruszcza, więc apeluję do panów ministrów o to, by w końcu wrócił do właściwej parafii. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stefana Wyszyńskiego w 40. rocznicę jego śmierci. Dokładnie dzisiaj mija 40 lat od śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia był wybitnym przywódcą duchowym, profesorem prawa kanonicznego, kapelanem polowym żołnierzy Armii Krajowej, dwukrotnym uczestnikiem konklawe, organizatorem pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i obchodów milenium chrztu Polski. Uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. Aresztowany przez władze komunistyczne i internowany przez 3 lata, opracował program odnowy życia religijnego w Polsce zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Wyszyński zostawił po sobie wielką spuściznę. Rozumiał, że wiary i polskości nie można od siebie oderwać. Był jednym ze współtwórców przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Bardzo dziękuję panu posłowi. Zapraszam teraz pana posła Janusza Korwin-Mikkego, Konfederacja.

Otóż chciałem oświadczyć, że nie zgadzam się na tryb, w jaki Sejm potraktował bardzo ważną sprawę, jaką było porwanie samolotu przez reżim jego ekscelencji Aleksandra Łukaszenki.

Nie każdy się musiał z tym zgodzić. Oczywiście tego typu wyczyn reżimu Łukaszenki musi być surowo ukarany. Przykładowo proponuję, żeby wszystkie państwowe samoloty i ciężarówki, pojazdy państwa białoruskiego były po prostu kontrolowane w każdym państwie przez kilka godzin pod kątem, czy nie zawierają np. bomby. Gdyby coś takiego robiono, toby reżim się czegoś być może nauczył. Natomiast wygłaszanie oświadczeń, niekoniecznie spójnych ze sobą, wypowiadanie tysięcy słów niczego nie zmienia. Reżim Łukaszenki przeżył już nie takie oświadczenia. Przecież nie to chodzi, żeby sobie pogadać, tylko o to, żeby tego typu poczynania były karane, bo jeżeli tego typu poczynania nie będą karane bardzo dotkliwie, to jutro reżim jego ekscelencji Mikołaja Maduro porwie samolot z Brazylii do Kolumbii, Izrael porwie samolot z Egiptu do Libanu, a Polska, jak dobrze pójdzie, porwie samolot z Niemiec na Ukrainę i dalej będziemy sobie to wszystko porywali.

Usiąść?

A chodziło o potępienie porwania samolotu. Niestety nie było tego widać po oświadczeniu sejmowym. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz panią poseł Agnieszkę Soin, Prawo i Sprawiedliwość, o wygłoszenie oświadczenia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Życzę wam wszelkiej pomyślności w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb mieszkańców, satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej, wielu dalszych sukcesów oraz nowych ambitnych wyzwań. Wasze zaangażowanie oraz ciężka praca przyczyniają się do wzmożonego rozwoju lokalnego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Pragnę serdecznie podziękować za wasz trud i poświęcenie, z jakim służycie naszemu społeczeństwu, oraz życzyć wam samych sukcesów. Bardzo dziękuję, pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 30. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny kolejnego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na dzień 15 czerwca 2021 r. zostanie paniom i panom posłom doręczony.